istotnym elementem w profilaktyce są prawidłowe wzorce stylu życia, profilaktyka pierwotna, czyli diagnozowanie, oraz już profilaktyka wtórna, ten następny etap.

Bardzo bym prosiła panią minister o udzielenie informacji w tym temacie. Dziękuję pięknie. Dziękuję, pani poseł, za zadanie pytania. Uprzejmie proszę panią sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefę Szczurek-Żelazko o udzielenie odpowiedzi. Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Zachodzące zmiany cywilizacyjne, zmiany demograficzne, zmiany stylu życia powodują wiele problemów zdrowotnych, które wymagają szczególnej troski rządu, ministra zdrowia. Z roku na rok zwiększają się nakłady na świadczenia profilaktyczne. Te nakłady znajdują się w różnych źródłach, m.in. Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach swojego planu finansowego uwzględnia środki na profilaktykę, na promocję zdrowia, na różnego rodzaju badania, które mają na celu wczesne wykrycie zmian, które mogą w przyszłości skutkować dużymi problemami zdrowotnymi. Ale również na ten cel przeznaczamy środki z budżetu państwa, będące w dyspozycji ministra zdrowia. Gros środków jest też przeznaczanych ze środków z Unii Europejskiej, będących w dyspozycji m.in. ministra zdrowia. Profilaktyka jest priorytetem. Coraz większą uwagę w Ministerstwie Zdrowia zwracamy na kreowanie programów profilaktycznych, wprowadzanie elementów profilaktyki do różnych obszarów funkcjonowania ochrony zdrowia, m.in. w ramach działań profilaktycznych przeprowadzamy badania na temat stanu zdrowia seniorów. Te badania. Będziemy mieli pełen obraz sytuacji już w roku 2020 w ramach badania PolSenior 2, w którym analizujemy stan zdrowia Polaków po 60. roku życia. Ale równolegle realizowane są zadania, tak jak wspomniałam, w ramach różnych programów.

Jest m.in. to cel piąty, który wskazuje na konieczność podejmowania działań z zakresu promocji zdrowia i aktywnego starzenia się. W ramach tego celu w tym roku przeznaczyliśmy ponad 8 mln zł. W ramach tego działania prowadzimy, realizujemy zadania kierowane do populacji powyżej 50. roku życia, m.in. związane ze szkoleniami z zakresu żywienia dostosowanego do indywidualnego stanu zdrowia, z profilaktyką występujących dolegliwości dietozależnych. Łącznie w tym roku z tych edukacyjnych działań skorzystało już ponad 840 osób w wieku akurat 50+. Są też szkolenia z zakresu aktywności fizycznej seniorów, które są realizowane w ramach projektów finansowanych przez Narodowy Program Zdrowia.

Na ten program przeznaczamy w tej perspektywie 225 mln zł. Celem tego programu jest osiągnięcie wskaźników umieralności na choroby nowotworowe porównywalnych z wskaźnikami z krajów z innego obszaru Unii Europejskiej czy też światowymi. W ramach tego programu realizujemy szereg badań przesiewowych, są to m.in. badania kolonoskopowe, finansowane z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia czy też budżetu państwa. Wykonano ponad 100 tys. badań tego typu w populacji, do której kierowane były te badania.

Przeprowadzane były też badania w kierunku wykrycia raka płuc przy użyciu niskodawkowej tomografii komputerowej. Ponadto prowadzimy szkolenia personelu medycznego, lekarzy, pielęgniarek, nie tylko onkologów, ale głównie onkologów.

W 2018 r. rozpoczęliśmy realizację zadania pn. „Ogólnopolski program badań przesiewowych” w kierunku tętniaka aorty jamy brzusznej. Na ten program m.in., tak jak powiedziałam, przeznaczyliśmy w ramach tych środków programu POLKARD ponad 21 mln zł. To nie tylko ten program, ale również wsparcie wielu podmiotów leczniczych, które realizują zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, m.in. doposażenie ich w niezbędny sprzęt do wczesnej diagnostyki. Kolejny program to jest program profilaktyki chorób naczyń mózgowych. Celem programu jest wzmocnienie świadomości w zakresie profilaktyki i wczesne rozpoznanie objawów chorób naczyń mózgowych. Oprócz tych działań, takich typowo profilaktycznych, jak badania, konsultacje, program ten obejmuje też edukację, przede wszystkim lekarzy, lekarzy rodzinnych, pielęgniarek rodzinnych w kierunku wczesnego wykrywania (Dzwonek) objawów tychże chorób. Następny program to jest program profilaktyki nowotworów szyi, głowy - ponad 6 mln zł.

Wysoka Izbo! Tak jak Ministerstwo Zdrowia podkreśla, profilaktyka jest przede wszystkim tańsza, za tym przemawia ekonomia.

Czy Ministerstwo Zdrowia ma dla tej grupy osób przygotowany program profilaktyczny?

Oczywiście jeżeli chodzi o profilaktykę, promocję zdrowia, propagowanie postaw prozdrowotnych, istotną rolę w tym zakresie odgrywają pracodawcy.

Obecnie jeżeli mówimy o życiu w zdrowiu, przeżywalności w zdrowiu kobiet, czyli bez ograniczonej sprawności, jest to wiek ponad 61 lat. Jeżeli mówimy o mężczyznach i ich przeżywalności w zdrowiu, czyli bez ograniczeń zdrowotnych, to są to 64 lata. Dlatego bardzo ważne jest motywowanie, stymulowanie pracodawców, aby zechcieli włączyć się w ten nurt profilaktyki, promocji zdrowia, propagowania aktywnego starzenia się poprzez realizację różnych programów. Między innymi Instytut Medycyny Pracy w Łodzi podejmuje działania edukacyjne pracodawców, kadry zakładów pracy, pracowników służb, przede wszystkim medycyny pracy w kierunku animacji przez nich programów promocji, aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania się. Takie programy są wspierane przez instytut, ale również jest możliwość pozyskania środków z różnych źródeł, m.in. Instytut Medycyny Pracy i Ministerstwo Zdrowia zorganizowały wspólnie z pracodawcami konkurs „PracoDawca Zdrowia”, w ramach którego ocenialiśmy działania pracodawców nakierowane na troskę o zdrowie pracowników. Wielu pracodawców włącza się aktywnie, organizując m.in. różnego rodzaju zajęcia z zakresu aktywizacji, promocji zdrowego stylu odżywiania, organizowania lunchboxów w zakładach pracy, gdzie promuje się zdrowe żywienie.

Dziękuję serdecznie, pani minister.

Proszę bardzo o zadanie pytania. Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! 20 listopada zapadł ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego działalności szpitali. Trybunał orzekł, że art. 59 ustawy o działalności leczniczej w zakresie, w jakim każe samorządom pokrywać straty szpitali, jest niekonstytucyjny. Trybunał zauważył, że finansowanie służby zdrowia jest zadaniem rządu i Narodowego Funduszu Zdrowia, a nie samorządów. Podkreślił, że środki przekazywane przez NFZ są zbyt małe, by pokryć koszty funkcjonowania szpitali. Dobrze wiemy, że sytuację w szpitalnictwie miała poprawić wprowadzona przez PiS sieć szpitali i formy płatności w postaci ryczałtów. Kolejki się wydłużają, zadłużenie szpitali rośnie, wszystko to uderza przede wszystkim w pacjentów. Pani Minister! W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego chciałam zadać pani pytanie. Macie 18 miesięcy na wdrożenie zmian. Chciałabym też wiedzieć, w jaki sposób Ministerstwo Zdrowia i NFZ zamierzają wesprzeć jednostki samorządowe, którym przyszło się zmierzyć z koniecznością uzupełnienia środków w kasie NFZ, a nie mają tak naprawdę żadnych dodatkowych środków na pokrywanie tego typu strat. Chciałam też zapytać, czy Ministerstwo Zdrowia zamierza zabezpieczyć w przyszłorocznym budżecie środki na odszkodowania dla samorządów, które w związku z wyrokiem wejdą na drogę sądową w celu odzyskania pieniędzy, które musiały zamiast NFZ-u przeznaczyć na uzupełnienie środków w podległej jednostce służby zdrowia. Proszę o odpowiedź panią minister. Wysoka Izbo! Kilka dni temu pojawiło się uzasadnienie tego wyroku, które jest przedmiotem szczegółowej analizy przeprowadzanej przez Departament Prawny w Ministerstwie Zdrowia. Jak państwo doskonale wiecie, w swoim wyroku trybunał wyznaczył czas na dostosowanie aktualnie obowiązujących przepisów na 18 miesięcy. Uzasadnienie dotarło do nas dopiero kilka dni temu.

Mamy świadomość, że należy to zmienić.

Pani poseł... ...z tytułu udziału w podatkach było ponad 200 mld zł, w tej chwili jest 251, więc te środki są w samorządach. Oczywiście zadaniem samorządów jest wspieranie podmiotów leczniczych, natomiast finansowanie stricte świadczeń jest rzeczywiście sprawą budżetów Narodowego Funduszu Zdrowia. Chciałabym państwu też przypomnieć, że z roku na rok wzrastają nakłady na ochronę zdrowia.

Jest to ewidentny wzrost, o ponad 30%, w przeciągu kilku lat. Pozwolicie państwo mi odpowiedzieć? Z roku na rok wzrastają przychody. Również w tym roku trzykrotnie był zmieniany plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia.

To są środki przekazywane konkretnie do podmiotów leczniczych. Jeżeli chodzi o koszty osobowe, bo państwo o to też pytacie, oczywiście z tytułu różnych ustaw zwiększają się koszty pracy, chociażby z powodu wzrostu płacy minimalnej czy też regulacji resortowych, np. ustawy o minimalnym wynagrodzeniu zasadniczym, jak również z powodu rozporządzeń ministra zdrowia, za sprawą których zwiększamy wynagrodzenie w poszczególnych grupach. Na te zadania zostały przekazane środki. W niektórych przypadkach, jeżeli chodzi o rozporządzenia, były to środki dedykowane, przekazane w pełni na wzrost wynagrodzeń. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku pielęgniarek, gdzie przekazujemy w 100% środki na podwyżki wynagrodzeń. I, co ciekawe, niektórzy pracodawcy tych środków nie wykorzystują. Również były przekazane dodatkowe środki na wzrost wynagrodzeń lekarzy, ratowników medycznych.

Chciałabym również podkreślić, że zadłużenie nominalnie rzeczywiście wzrasta, natomiast jeżeli porównamy to do wzrostu przychodów, to de facto jest to mniejsze proporcjonalnie zadłużenie niż było w poprzednich latach. Mało tego, okazuje się, że wpływ na wyniki finansowe podmiotów leczniczych ma też jakość zarządzania. Szanowni państwo, 8% podmiotów leczniczych w Polsce generuje 80% zobowiązań, 73% podmiotów leczniczych się bilansuje. Czyli może też z drugiej strony należy zwrócić na to uwagę - 73% podmiotów leczniczych się bilansuje, to są dane twarde, wynikające ze sprawozdań finansowych. W Ministerstwie Zdrowia podejmujemy konkretne działania w celu ujednolicenia chociażby rachunku kosztów, metod porównywalności pewnych rodzajów kosztów. Są pewne mechanizmy, które pozwolą zoptymalizować koszty: koncentracja świadczeń, koncentracja zamówień publicznych. To są elementy sprawnego zarządzania stosowane w gospodarce rynkowej. Myślę, że one też winny mieć zastosowanie w ochronie zdrowia. Nie tylko myślę, ale tak powinno być. Oczywiście analizujemy sytuację, z troską pochylamy się nad tym, zwiększamy z roku na rok nakłady na ochronę zdrowia. Ustawa 6-procentowa (Dzwonek), gwarantująca 6% produktu krajowego brutto w 2024 r., jest dowodem na to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości traktuje służbę zdrowia priorytetowo. Dziękuję, pani minister, za odpowiedź. Nie chcę być złośliwy, bo nigdy w życiu nie byłem złośliwy, ale z tego, co pani minister mówi, niedługo z przyjemnością będziemy chodzili do lekarzy. To dobrze.

Pani minister była zobowiązana do rzetelności, a pani zmanipulowała. Algorytm dotyczący 6%.

To są manipulacje.

I chcemy powiedzieć pani, że manipuluje pani również informacjami.

O co nam chodzi? O samorządy, które muszą płacić więcej. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nie zmieniła się. A ceny prądu państwo nie zmienili, podwyższacie ją. Mówimy o klapie. Na Kurskiego, na telewizję publiczną są pieniądze, na szpitale nie ma pieniędzy. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę panią minister o odpowiedź.

Szanowny Panie Marszałku! No cóż, pani poseł nie przekonam, bo już wielokrotnie próbowałam pani przedstawiać fakty, fakty które wynikają z planów Narodowego Funduszu Zdrowia, z odpowiednich pozycji w budżecie państwa. Natomiast jeżeli chodzi o ustawę 6-procentową, to jest to jedyna tego typu ustawa podjęta właśnie przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, która wskazuje konkretną drogę dojścia do poziomu, który gwarantuje poprawę jakości udzielania świadczeń. Oczywiście to nie jest jeszcze ideał, do którego dążymy, i w kolejnych latach na pewno będziemy podejmować działania, aby poprawić tę sytuację. Natomiast fakty są takie, że w 2019 r. wydajemy 4,86% produktu krajowego brutto. W 2020 r. wydamy 5,03% produktu krajowego brutto.

Takie są fakty uwidocznione zarówno w planach finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia, jak również w budżecie państwa, ponieważ tam też znajdują się środki na ochronę zdrowia. Natomiast jeszcze jedną rzecz chciałabym wspomnieć. Rząd wspiera również w inny sposób podmioty lecznicze, chociażby gwarantując środki na inwestycje po to, aby szpitale nie musiały własnych środków z dochodów na świadczenie usług przeznaczać na inwestycje. W tej perspektywie, w ostatniej perspektywie finansowej wydaliśmy na ten cel 15 mld zł. To jest ta kwota, która zasiliła infrastrukturę szpitali poprzez właśnie różnego rodzaju kanały, m.in. w Ministerstwie Zdrowia. Finansowaliśmy doposażenia szpitali pediatrycznych wysokospecjalistycznych, onkologicznych, kardiologicznych, jak również szpitalnych oddziałów ratunkowych.

Tak więc działania są sukcesywnie podejmowane.

Wynikiem są dłuższe kolejki, pani minister, a pieniądze do narodowego funduszu płacą ludzie, a nie państwo. Pani posłanka Marcelina Zawisza z klubu parlamentarnego Lewica postanowiła zadać pytanie w sprawie zasad kontraktowania usług oddziałów położniczych w Polsce. Na pytanie będzie odpowiadała pani minister. Pani posłanka ma 2 minuty na zadanie pytania. Zapraszam. Wysoka Izbo! Szanowna Pani Minister! Tego, ile razy podkreślali państwo, że mają na uwadze dobro rodziny, matki, a ostatnio nawet, jak usłyszeliśmy w exposé premiera, kobiety, nie jestem w stanie zliczyć. Premiowane miałyby być oddziały większe, odbierające ponad 400 porodów rocznie.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania.

Jakie są projektowane warunki dotyczące minimalnej odległości między oddziałami położniczymi, umożliwiające uzyskanie projektowanej przez NFZ premii?

Jak rząd, likwidując porodówki, chce zapewnić bezpieczeństwo kobietom w ciąży, rodzącym, noworodkom, szczególnie wcześniakom i dzieciom wymagającym natychmiastowej pomocy medycznej? Niedofinansowanie szpitali i brak lekarzy i lekarek powodują zamykanie porodówek w całej Polsce.

Ile środków ministerstwo planuje przeznaczyć na kampanię informacyjną mającą na celu poinformowanie obywateli i obywatelek, które porodówki zostaną zamknięte? Dziękuję pani posłance Marcelinie Zawiszy z klubu Lewica. Proszę o odpowiedź panią minister. Uprzejmie proszę. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Opieka nad kobietą ciężarną, kobietą rodzącą jest w obszarze wyjątkowej troski ministra zdrowia, a dowodem na to są m.in. regulacje, które zostały wprowadzone. Wprowadziliśmy m.in. standard organizacyjny opieki okołoporodowej, który wyraźnie definiuje, jakie świadczenia są należne kobiecie ciężarnej, jak również w trakcie porodu. Ponieważ z tego tytułu było wiele nieporozumień, minister zdrowia podjął decyzję o opracowaniu tego standardu. Ten standard został wdrożony i jest realizowany zarówno przez położne środowiskowo-rodzinne, lekarzy ginekologów, położników, jaki i w ramach opieki szpitalnej w oddziałach ginekologicznych czy też ginekologiczno-położniczych w szpitalach.

Coraz częściej mówi się o problemie depresji u kobiet ciężarnych, po porodzie. W związku z tym wprowadziliśmy jako obligatoryjne świadczenie diagnozowanie wstępnych objawów depresji i udzielanie wsparcia w tym zakresie. Jak państwo wiecie, kontraktowanie świadczeń odbywa się w sposób dwojaki. Po pierwsze, na podstawie ryczałtów, które są przeznaczane dla szpitali objętych siecią szpitali. Chciałabym w tym miejscu podkreślić, że wprowadzenie sieci szpitali po raz pierwszy zagwarantowało szpitalom stabilizację, ponieważ w procedurze kontraktowania 3-letniego w trybie konkursowym żaden szpital nigdy nie miał pewności, czy świadczenia wszystkich oddziałów zostaną zakontraktowane. Taka sytuacja miała miejsce. Mogłabym podać przykłady z mojego terenu, gdzie nie zostały zakontraktowane z dnia na dzień świadczenia oddziałów czy np. zespołów ratownictwa, bo wszedł zupełnie inny, często komercyjny, podmiot. Dlatego wprowadziliśmy sieć szpitali, żeby zagwarantować szpitalom stabilizację w postaci kontraktu w perspektywie co najmniej 10-letniej.

Rzeczywiście część tych szpitali wykonuje bardzo dużo tego typu świadczeń, ale są szpitale, które realizują np. 64 porody rocznie, 74 porody rocznie czy 150 porodów rocznie. Szanowni państwo, ilość wykonanych świadczeń jest gwarancją jakości i to jest oczywista rzecz, a pochodną tego jest opłacalność ekonomiczna, ale najważniejsza jest jakość. Dlatego też rozważa się to, czy ewentualnie nie premiować dodatkowo tych świadczeniodawców, którzy wykonują dużą ilość procedur, bo w tym momencie jest zagwarantowana jakość.

Natomiast na dzień dzisiejszy nie ma w tym zakresie żadnego zarządzenia prezesa, a, jak państwo wiecie, na podstawie zarządzenia prezesa następuje zmiana sposobu finansowania.

Dziękuję serdecznie, pani minister. Pytanie dodatkowe zada pani posłanka Marcelina Zawisza. Odniosła się pani tutaj do standardów, jakie są w Polsce odnośnie do porodów. Chciałam zapytać, czy ministerstwo jest świadome tego, że, jak pokazuje badanie Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, wśród kobiet, które rodziły drogami naturalnymi, 43,4% miało wywoływany poród, 60% podaną kroplówkę z oksytocyną i tylko 38,5% kobiet miało zapewniony złoty standard, czyli kontakt z dzieckiem minimum 2 godziny po porodzie. Mam pytanie, czy ministerstwo w ogóle ma świadomość tego, jak wygląda w Polsce sytuacja na porodówkach.

Dziękuję serdecznie pani posłance. Zapraszam panią minister. Wysoka Izbo! Standard opieki okołoporodowej został wprowadzony dopiero kilkanaście miesięcy temu, w związku z czym analizujemy na bieżąco efekty, skuteczność działania tego standardu. Zgodnie z ustawą instytucją, która ma oceniać wdrażanie standardów w poszczególnych podmiotach leczniczych, jest Narodowy Fundusz Zdrowia oceniający również jakość udzielanych świadczeń.

Tak jak powiedziałam, monitorujemy sytuację, podejmujemy działania korygujące.

Cenimy sobie bardzo tę współpracę i spotykamy się regularnie po to, aby lepiej wdrożyć, implementować w obszarze ochrony zdrowia właśnie ten standard.

W szpitalach jest to ważny element rozwoju dziecka, zachowania dobrostanu matki. W związku z tym minister zdrowia podjął decyzję o dodatkowym finansowaniu m.in. tego szczególnego obszaru, jakim jest żywienie kobiety ciężarnej. Ostatnio, jak państwo wiecie, na posiedzeniu Rady Ministrów została przyjęta ustawa, która gwarantuje bezpłatne leki dla kobiet w ciąży.

One stanowią ważną pozycję w wydatkach, w budżetach domowych rodzin, dlatego minister zdrowia, premier Mateusz Morawiecki podjęli decyzję o wspieraniu chociażby nawet tego obszaru. Dziękuję bardzo, pani minister.

A na to pytanie postanowił odpowiedzieć podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu pan minister Sławomir Mazurek. Bardzo proszę, panie pośle. Ma pan 2 minuty na zadanie pytania. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w skrócie zwana BDO, jest systemem informatycznym utworzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Integralną częścią BDO jest rejestr podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który to rejestr został uruchomiony 24 stycznia 2018 r. Od 1 stycznia 2020 r. planowane jest uruchomienie kolejnych modułów systemu, to jest modułu ewidencji i modułu sprawozdawczości. Obowiązek ewidencji w internetowej bazie danych rodzi wiele problemów, gdyż osoby zobowiązane do rejestracji w systemie niewiele wiedzą o tym systemie, nie mają pełnej wiedzy. Ponadto problem dotyczy braku jasnych zasad, określających, kto ma się rejestrować w bazie danych o odpadach BDO i ewidencjonować to, co jest wyrzucane jako odpad. Dodatkowo wprowadza obowiązek określania rodzajów odpadów.

Dlatego zadaję pytanie. Ilu przedsiębiorców dotychczas zarejestrowało się w systemie, panie ministrze? Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie panu posłowi. Proszę o zajęcie stanowiska i odpowiedź pana ministra Sławomira Mazurka. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie i Panowie Posłowie! Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów spoczywa na przedsiębiorcach od roku 2001, zatem 1 stycznia nie wprowadzamy żadnych nowych obowiązków. Przepisy dotyczące ewidencji i sprawozdawczości nie zmieniają się. Jedyna zmiana dotyczy zastąpienia dotychczasowej formy papierowej dokumentów z zakresu gospodarki odpadami formą elektroniczną. To stanowić powinno ułatwienie dla przedsiębiorców. Jednocześnie wychodzimy naprzeciw tym wszystkim przedsiębiorcom, którzy zgłaszali do nas uwagi o dopuszczenie równoległego funkcjonowania bazy, i takie zapisy zostaną przedstawione do realizacji.

W roku 2015 pojawiła się propozycja przetargu, niestety nie były gotowe rozporządzenia, żeby ten przetarg przeprowadzić, on by się nie powiódł. Dlatego też ostatecznie bazę danych przygotował Instytut Ochrony Środowiska w drodze powierzenia in-house. Harmonogram został dotrzymany, baza jest przygotowana. Mogą oni dokonywać tam szeregu działań. Oczywiście wszystkie funkcjonalności będą mogły być uruchomione zgodnie z ustawą, bo baza, jej zakres dotyczy tego, co jest w ustawie. Zgodnie z ustawą, która była w połowie ostatniego roku nowelizowana, te funkcjonalności, te kolejne moduły. To metoda zwinna, taka metoda, przy pomocy której administracja stara się wykonywać kolejne moduły, czyli moduł po module, gdzie przyjmuje się pewne założenia, potem dokonuje się sprawdzeń, pracują zespoły analityczne, ostatecznie jest to przygotowywane do wytworzenia w zespołach produkcyjnych. Zgodnie z tą metodyką, także z metodyką Prince, ten projekt był prowadzony. Integralną częścią BDO jest rejestr podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Liczba podmiotów znajdujących się obecnie w rejestrze BDO to ponad 165 tys.

Pragnę wyraźnie powiedzieć, że te wszystkie podmioty gospodarcze, które do tej pory nie prowadziły ewidencji zgodnie z ustawą z 2001 r., nie są zobowiązane do tego, aby się rejestrować w bazie danych odpadowych. Jedynym wyjątkiem są tutaj podmioty, które oferują torby plastikowe, zgodnie z dyrektywą, które muszą być objęte opłatą, więc ta możliwość sprawozdawczości elektrycznej to jest jedyne novum.

Jest to wszystko gotowe, po wszelkich testach. Tutaj mamy szansę na kompleksowe gromadzenie, zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami. Zapewni to podmiotom w pełni elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencji i sprawozdawczości. Do tej pory było to robione jedynie przez urzędy marszałkowskie, które musiały to ręcznie wpisać. Dzisiaj będzie można robić to przez bazę. Analiza i ocena danych umożliwi prowadzenie diagnozy stanu gospodarki odpadami, ocenę i prognozowanie trendów. Przed nami wprowadzenie rozszerzonej gospodarki odpadami. Dobrze mieć pełną wiedzę o tym, ile odpadów wytwarzamy i w jaki sposób one migrują po Polsce.

Na pewno Inspekcja Ochrony Środowiska, która jest organem kontrolnym, będzie pomagać wszystkim podmiotom.

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu ministrowi. Dziękuję za tę informację.

Prawdopodobnie ci przedsiębiorcy obawiają się tego, są zaniepokojeni.

To jest jedno moje pytanie.

Szanowni Państwo!

Ona nam wygenerowała duże zainteresowanie na infoliniach, jeśli chodzi o pytania, ale dała też szansę na wykazanie się rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców, który interweniował w tej sprawie, aby poza tym, co jest w ustawie, dokonać takiego objaśnienia w przypadku wszystkich przedsiębiorców, żeby to, o czym powiedziałem w pierwszej części mojego wystąpienia, przyjęło formę takiego objaśnienia zgodnie z konstytucją dla biznesu, z art. 33 tej konstytucji, która wskazuje z jednej strony, żeby wszelkie wątpliwości rozstrzygać na korzyść przedsiębiorcy, a z drugiej strony daje możliwość przygotowania specjalnych objaśnień, które wskazują, kto takiemu obowiązkowi podlega. Tu jest pewna trudność, jeśli chodzi o szacowanie wszystkich podmiotów. To rynek dynamiczny, on się zmienia, część podmiotów wypada, powstają nowe podmioty. Szacowaliśmy, że tych podmiotów może być więcej. Zakładamy, że ta liczba 160 tys. nie będzie drastycznie rosnąć.

Mówiłem o inspekcji. Wpisanie się do bazy zajmuje kilka minut, więc nie ma problemu.

Witam i pozdrawiam dzieci na galerii. O, jak ładnie. Proszę państwa, pan poseł Czesław Hoc z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość chciałby w swoim imieniu oraz w imieniu nieobecnych posłów Leszka Dobrzyńskiego, Artura Szałabawki, Michała Jacha, Małgorzaty Golińskiej i pana Pawła Szefernakera zadać pytanie w sprawie propozycji likwidacji opłaty uzdrowiskowej w gminach uzdrowiskowych zawartej w „Białej księdze regulacji systemu promocji turystycznej w Polsce” Na to pytanie odpowie podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju pan minister Marek Niedużak. Panie pośle, proszę o zadanie pytania. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Pani Ministrze! Wysoka Izbo!

Dlatego że kilka tygodni temu ukazała się na zamówienie Ministerstwa Sportu i Turystyki, dawnego Ministerstwa Sportu i Turystyki „Biała księga regulacji systemu promocji turystycznej w Polsce”

Jest propozycja likwidacji opłaty uzdrowiskowej. Ja tylko przypomnę albo podkreślę, że np. największe uzdrowisko w Polsce, czyli Kołobrzeg, Wenecja Północy, w poprzednim roku uzyskało z tego tytułu 33 mln zł. Konstrukcja tej opłaty jest następująca: że połowę tych środków uzyskuje się z tytułu opłat wczasowiczów i turystów, a połowę z budżetu centralnego. Dziękuję serdecznie. Proszę, panie ministrze. Wysoka Izbo! Dziękuję. Panie Pośle! Mógłbym też bardzo krótko, bo to jest bardzo konkretne pytanie: tak, nie. Ja też mogę odpowiedzieć bardzo krótko: nie ma takich planów. Bo chciałem dwa zdania uzasadnienia.

To materiał do dyskusji i analiz. Nie ma planów likwidacji opłaty. Panie marszałku, lapidarne ujęcie, treściwe, zasadne. Dziękuję wam serdecznie. Idziemy dalej. Posłanki Małgorzata Tracz, Urszula Zielińska i Agnieszka Pomaska oraz posłowie Bartłomiej Sienkiewicz i Tomasz Aniśko postanowili zadać pytanie w sprawie celu polegającego na osiągnięciu przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz działań rządu RP związanych z jego realizacją. Na to pytanie będzie odpowiadał podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu pan minister Sławomir Mazurek. Zapraszam panią posłankę Małgorzatę Tracz do zadania pytania. Proszę bardzo. 2 minuty, pani posłanko. Uczę się powoli, ale już się nigdy nie pomylę. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Tydzień temu premier Morawiecki ogłosił rzekomy gigantyczny sukces. Ten rzekomy sukces miał polegać na tym, że Polska uzyskała zwolnienie z osiągnięcia unijnego celu neutralności klimatycznej w 2050 r. W okrągłych słowach wmawiano nam, że wynegocjowane zapisy zwiększą szansę Polski na uzyskanie realnych, konkretnych pieniędzy z funduszu sprawiedliwej transformacji oraz Europejskiego Banku Centralnego i że wynegocjowane zwolnienie będzie przyczyniało się do poprawy jakości życia polskiej rodziny. Chciano nas przekonać, że rząd prowadzi ambitną, a jednocześnie racjonalną politykę klimatyczną i energetyczną, politykę rzekomo najlepszą, dostosowaną do potrzeb Polski i polskiego społeczeństwa. Naprawdę myślicie, że ktoś się na to nabierze? Na tę demagogię? Bo to jest czysta demagogia, a nie żadna strategia. Ta decyzja była dobitnym przykładem na to, że ten rząd prowadzi krótkowzroczną politykę braku ambicji, politykę kosztem przyszłości i bezpieczeństwa naszych dzieci i wnuków, politykę kosztem polskiej gospodarki. Ta decyzja pozostawia Polskę, jedyny kraj, który zanegował politykę klimatyczną Europy, bez europejskiego wsparcia politycznego czy finansowego, bez szans na godny udział w funduszu sprawiedliwej transformacji i 100-miliardowym budżecie, który Unia Europejska przeznaczy na to zadanie. Dziś w polityce klimatycznej i energetycznej rządu brak ambicji i celu. Po pierwsze: Czy rząd planuje wyznaczyć jakąkolwiek datę osiągnięcia przez Polskę neutralności klimatycznej? Jeśli tak, to jaką? Kolejne: Na jakim etapie jest opracowywanie nowej wersji zintegrowanego krajowego planu na rzecz energii i klimatu do 2030 r. Czy zmiany będą uwzględniały zalecenia Komisji Europejskiej i zostaną przysłane do niej na czas?

Dziękuję pani posłance Małgorzacie Tracz. Zapraszam pana ministra Sławomira Mazurka. Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego prowadzi racjonalną politykę klimatyczno-energetyczną, politykę na miarę dążeń, nie tylko Unii Europejskiej, ale wszystkich, którzy uczestniczą w konwencji klimatycznej. To polski minister był prezydentem konferencji klimatycznej, to szczyt w Katowicach zakończył się wielkim sukcesem wspólnoty międzynarodowej i multilateralizmu. Więc ambicji nam nie brakuje, ale nie brakuje nam też racjonalnych argumentów, żeby prowadzić to w sposób zrównoważony, tak aby - o czym mówi Organizacja Narodów Zjednoczonych - nie powodować dodatkowo wykluczenia społecznego, żeby nikt nie pozostał z tyłu i żeby też wykorzystać synergię wszystkich trzech konwencji, z Rio, konwencji klimatycznej o ochronie bioróżnorodności i przeciwdziałaniu pustynnieniu. To rząd pani premier Beaty Szydło osiągnął sukces także w Paryżu, gdzie podpisano porozumienie paryskie, którego Polska jest członkiem. Polska zobowiązała się do osiągnięcia neutralności klimatycznej w drugiej połowie wieku zgodnie z zapisami Porozumienia paryskiego. Ale Polska jest też aktywnym członkiem Unii Europejskiej i bierze aktywny udział we wszystkich forach, które się polityką klimatyczną, energetyczną, a także synergią z innymi wyzwaniami, megatrendami jak osiągnięcia w zakresie tego, co jest. Także w nowym zielonym ładzie, czyli to, co dotyczy gospodarki obiegu zamkniętego, to także jest element i te synergię także będziemy chcieli budować. Starając się odpowiadać krócej na pani konkretne pytania, pragnę powiedzieć, odnieść się może jednak do tego, co pani powiedziała na początku, a co u mnie widniało jako ostatnie pytanie, czyli do tego, co wydarzyło się w trakcie spotkania Rady Europejskiej. Równocześnie zdecydowała, że Polska zostanie zwolniona z osiągnięcia już w 2050 r. neutralności klimatycznej. Polska będzie mogła rozwijać się w swoim tempie. Bo też nasza sytuacja jest daleko inna niż krajów Europy Zachodniej, jeśli chodzi o nasz miks energetyczny, jeśli chodzi o kapitał, którym dysponujemy. Nie chcemy doprowadzić do takiej sytuacji jak we Francji, do masowych protestów społecznych. Chcemy, żeby nasza droga do neutralności klimatycznej była drogą zrównoważoną, uwzględniającą wszystkich.

Warto też podkreślić, że koszty ewentualnego osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Polskę są znacznie wyższe niż średnia unijna i mogą oznaczać konieczność dodatkowych inwestycji rzędu 1–3% PKB. Nie oznacza to, że Polska nie będzie podejmować działań zmierzających do transformacji niskoemisyjnej. Polska, tak jak powiedziałem, jako strona porozumienia paryskiego jest zobowiązana do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Będziemy dochodzić do niej w swoim tempie, zgodnie z porozumieniami paryskimi. Nie blokowaliśmy jednocześnie ambicji innych państw członkowskich, które uważają, że mogą osiągnąć neutralność klimatyczną, mają też inny miks, mają elektrownie jądrowe, których my przez 30 lat nie zbudowaliśmy, a moglibyśmy sięgnąć jeszcze dalej.

Od wielu tygodni Polska pozostaje w dialogu z Komisją Europejską w sprawie kryteriów wsparcia oraz potrzeby objęcia przyszłym mechanizmem regionów i sektorów najbardziej narażonych na niekorzystne skutki transformacji. Rada potwierdzi takie podejście i będzie w dalszym ciągu negocjować jak najkorzystniejsze dla Polski warunki przyznawania środków.

Obserwujemy przecież ekstremalne zjawiska pogodowe, obserwujemy susze, obserwujemy nawalne deszcze. Tu też jest konieczne wprowadzenie adaptacji do zmian klimatu. Nie możemy jednak zapominać, że w naszym przekazie ta niezbędna transformacja energetyczna może prowadzić do większych kosztów dla obywateli. Dlatego też rzetelnie należy przekazywać informacje o kosztach i korzyściach z osiągnięcia neutralności klimatycznej. Chcielibyśmy uniknąć, tak jak powiedziałem wcześniej, tych sytuacji, które miały miejsce we Francji. Krajowy plan na rzecz energii i klimatu został rozpatrzony przez komitet europejski i zostanie on przedłożony Komisji Europejskiej zgodnie z planem. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie ministrze. Bardzo proszę pana posła Bartłomieja Sienkiewicza o zadanie pytania dodatkowego. Mamy do czynienia z przedstawicielem Ministerstwa Klimatu, które na razie zajmuje się również śmieciami i dzikiem. To jest najlepsze podsumowanie tego, jak państwo się tym klimatem zajmujecie. Nierozdzielone funkcje ministerstwa środowiska i Ministerstwa Klimatu powodują, że z jednej strony przedstawiciel rządu mówi o trosce o klimat, z drugiej strony płynnie przechodzi do śmieci, a jeszcze mamy dzisiaj w Sejmie rozmowę o wybijaniu dzików.

Panie ministrze, proszę. Panie Marszałku! Panie Pośle! Myślę, że kwestia śmieci jest ważna, szczególnie że staramy się kamieni kupę uprzątnąć, tak aby Polska się dynamicznie rozwijała, i bym tego nie trywializował. Ale chcę wyraźnie powiedzieć, że jeśli chodzi o kwestię planowania, przygotowywania tego wszystkiego, co dotyczy neutralności klimatycznej, tego, co dotyczy rozwoju także w zakresie neutralności klimatycznej, my staramy się to robić i robimy to, dla nas to jest bardzo istotne. Rozwijamy to, co dotyczy energetyki prosumenckiej. Program „Mój prąd” to jest program, który pozwala Polkom i Polakom na to, by instalować panele fotowoltaiczne. To wszystko, co dotyczy tego, z czym też wiąże się neutralność klimatyczna, w zakresie odnawialnych źródeł energii, to jest jeden z elementów właśnie neutralności klimatycznej. Dziękuję bardzo za tę opinię z sali. Jednocześnie program „Czyste powietrze” daje szansę na głęboką termomodernizację, wymianę źródła ciepła na bardziej ekologiczne. Myślę, że żaden rząd w historii nie wykonał i nie przygotował takich programów, które pozwalają nie tylko wybranym grupom społecznym czy instytucjom publicznym, ale także obywatelom na to, aby mogli do tej neutralności klimatycznej dążyć, aby mogli także wykorzystywać to, co daje nowoczesna technologia, w zakresie ogrzewania, w zakresie wytwarzania energii elektrycznej. Ale oczywiście neutralność klimatyczna to nie tylko prosument - to także to wszystko, co czeka nas w obszarze rolnictwa, w obszarze transportu. Stąd dla Ministerstwa Klimatu bardzo ważnym elementem jest promowanie i rozwijanie niskoemisyjnego transportu, elektromobilności. Na tym też się będziemy skupiać w naszych pracach. Jednocześnie to wszystko, co wiąże się z tymi zadaniami, chcemy pokazywać także jako narodowy wkład do tego, aby tę neutralność klimatyczną rozwijać, dobrze się do tego przygotować, tak aby faktycznie wykorzystać to do rozwoju kraju. Oczywiście dynamiczne dążenie, takie nieplanowane może być zagrożeniem dla rozwoju gospodarczego, ale dobrze przygotowane, w oparciu o jak najlepszą wiedzę, jest pewną szansą. Myślę, że w Ministerstwie Klimatu tę szansę będziemy chcieli pokazywać i wykorzystywać to wszystko po to, abyśmy mogli się rozwijać i te wieloletnie zapóźnienia w obszarze zmniejszania presji na środowisko zmniejszać.

Proszę bardzo panią poseł Teresę Wargocką o zadanie pytania. Dziękuję, panie marszałku. Badanie PISA organizuje międzynarodowe konsorcjum nadzorowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz przedstawicieli państw członkowskich. To największe badanie umiejętności uczniów na świecie. Badane są umiejętności w zakresie czytania ze zrozumieniem, rozumowania w naukach przyrodniczych oraz rozumowania matematycznego. Polską edycję tego badania prowadzi zespół Instytutu Badań Edukacyjnych. Badanie pokazuje poziom i zróżnicowanie umiejętności 15-latków, umiejętności, które rozwijane są w trakcie edukacji szkolnej oraz poza szkołą.

Pani Minister! Jaki jest poziom umiejętności kluczowych dla przyszłości młodego pokolenia Polaków w badanych obszarach na tle innych państw biorących udział w badaniu? Dziękuję serdecznie. Na pytanie odpowie sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pani minister Marzena Machałek. Bardzo proszę. Dziękuję. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rzeczywiście badanie PISA to bardzo ważne badanie międzynarodowe, które angażuje coraz więcej krajów na świecie i, co należy podkreślić, służy przede wszystkim oszacowaniu kompetencji uczniów 15-letnich w zakresie czytania, matematyki i nauk przyrodniczych. Jest cennym źródłem informacji na temat tych umiejętności, a także innych kontekstowych uwarunkowań, które powstawaniu, tworzeniu czy doskonaleniu tych umiejętności służą. I rzeczywiście warto podkreślić, że polscy uczniowie wypadli dużo lepiej w tym badaniu niż w 2015 r. Pamiętamy, że we wszystkich dziedzinach w tym badaniu była kilkunastopunktowa różnica w stosunku do poprzedniego badania, czyli nie dość, że mamy progres, to widać naprawdę duże „odbicie się” uczniów, jeśli chodzi o problemy, które wyniknęły w 2015 r. Najlepsze nasze wyniki oczywiście znajdują się w światowej czołówce i są powyżej średniej w OECD. Najlepsze wyniki w tym badaniu osiągnęli uczniowie z czterech regionów: Chin, Hongkongu, Singapuru i Makao. W rozumowaniu matematycznym polscy uczniowie wyprzedzają w Unii Europejskiej wszystkich poza młodymi Estończykami, w rozumieniu tekstu polska młodzież zajmuje czwarte miejsce wśród krajów Unii, w rozumowaniu w naukach przyrodniczych jest na trzeciej pozycji. Tu, jak pani poseł podkreśliła, była dobrana grupa badawcza, grupa uczniów spośród wielu, był to proces podwójnego losowania. Wydaje się, że to jest bardzo reprezentatywne badanie. I teraz to, co trzeba podkreślić - badanie PISA to badanie umiejętności, a nie systemów edukacji.

To jest istotne i to należy podkreślić.

Kolejny mówi o tym, gdzie uczniowie mogą uzyskać sukces dotyczący równości szans w edukacji ze względu na czynniki społeczne, i o tym, jakie znaczenie dla szkolnego życia, dla uczniów mają takie rzeczy, jak klimat szkoły, postrzeganie pracy nauczycieli, relacje uczniowskie, poczucie jakości życia uczniów, przekonania rodziców na temat własnych możliwości rozwojowych dzieci oraz zaangażowanie rodziców w edukację. Innymi słowy, badania PISA to nie tylko wyniki dotyczące tych umiejętności, ale też przyglądanie się, czy są nierówności społeczne, jaka jest jakość życia uczniów, dobrostan, jakie są kompetencje psychospołeczne, style pracy nauczycieli, postawy społeczne wobec uczniów oraz plany i aspiracje zawodowe.

Chcę też jasno podkreślić, że warto by tutaj zwrócić uwagę, bo o tym nie mówiliśmy, że w Polsce istnieją jeszcze relatywnie duże nierówności społeczne, jeśli chodzi o edukację.

To też jest ciekawe. Im większe poczucie przynależności, tym gorszy wynik.

Mamy oczywiście najniższy odsetek uczniów z najniższymi umiejętnościami i bardzo wysoki odsetek uczniów z wysokimi umiejętnościami, ale jeśli uczniowie już są w tej grupie o najniższych umiejętnościach, to trudno im z niej wyjść. Dziękuję, pani minister. Proszę. Pani Minister! Badanie, o którym mówimy, pokazuje poziom i zróżnicowanie umiejętności piętnastolatków m.in. w dziedzinie rozumowania matematycznego. I rzeczywiście tutaj jest powód do dumy, bo na tle krajów europejskich prezentujemy się doskonale. Lepsi są tylko Estończycy i Holendrzy. Ale chciałbym pokazać inną sytuację. Mianowicie ci, którzy poddawani są badaniu PISA, po kilku latach przystępują do egzaminu maturalnego z matematyki. I tu okazuje się, że matematyka to ich pięta achillesowa i przyczyna wielu niepowodzeń maturalnych. 8% licealistów i 16% uczniów techników tej matematyki nie zdaje. Co takiego się dzieje, że uczniowie, którzy świetnie rozumują matematycznie, wykładają się, mówiąc kolokwialnie, na maturze z matematyki i jak temu zaradzić? Pani minister, proszę.

Jego nauczanie miało niższą rangę, bo nie był to przedmiot obowiązkowy na maturze.

Chciałabym jasno powiedzieć, że jesteśmy na etapie badań kontekstowych i uwarunkowań oraz dyskusji i analizy tych badań kontekstowych i dzisiaj nie można powiedzieć, że dane zbierane w ramach PISA pozwalają na jednoznaczne wskazanie przyczyn średniego konkretnego wyniku dla danego kraju. Próba interpretacji każdorazowo wymaga przyglądaniu się kontekstowi kraju. Chciałabym to bardzo jasno powiedzieć. A z matematyką mamy jeszcze dużo pracy, też nad metodą uczenia matematyki, nad przygotowaniem i doskonaleniem nauczycieli.

To wszystko jest dla nas dużym i cennym źródłem informacji, natomiast takich badań dotyczących uczniów, którzy zdają maturę, które by tak kompleksowo pokazywały nas na tle innych krajów, nie mamy, więc nie będę tutaj w sposób jednoznaczny mówiła o tym, co jest tu przyczyną, bo to nie jest jedna kwestia.

Dlatego my też bierzemy to pod uwagę, tak jak to już mówiłam, w tworzeniu takiego horyzontalnego dokumentu, jakim jest Zintegrowana Strategia Umiejętności. Sensowne jest dyskutowanie o wielu czynnikach warunkujących zmiany wyników, ale gdybyśmy pytali, dlaczego mamy tak dobre wyniki, co na to wpłynęło, to chodzi tu o to, co podkreśla też OECD, że wyniki we wszystkich krajach są skorelowane mocno z rozwojem gospodarczym. Im bogatszy kraj, tym lepsze wyniki. Pozytywne zmiany gospodarcze w Polsce sprzyjają dobrym wynikom edukacyjnym poprzez podniesienie jakości życia. Polityka społeczna ostatnich lat, transfery społeczne pomogły w osiąganiu lepszych wyników (Dzwonek), szczególnie przez uczniów z najbiedniejszych rodzin. Przed nami oczywiście dużo pracy, by te wyniki były coraz lepsze. Budowanie odpowiedzialnej strategii umiejętności i odpowiedzialne wykorzystanie tych środków unijnych w kolejnej perspektywie - przed nami. Dziękuję serdecznie, pani minister. Witam panią posłankę Monikę Rosę, panią posłankę Izabelę Katarzynę Mrzygłocką, pana posła Michała Szczerbę, którzy zadadzą pytania w sprawie lawinowo rosnącej liczby nielegalnie działających placówek zapewniających całodobową opiekę osobom przewlekle chorym, niepełnosprawnym i w podeszłym wieku. Na te pytania odpowie pan minister Marcin Zieleniecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pan poseł Michał Szczerba. Tak mam podane. Tak państwo ustaliliście, ale jeżeli chcecie się zamienić, zamieńcie się. Wysoka Izbo! Polskie społeczeństwo się starzeje, ale również chcemy dzisiaj zwrócić uwagę Wysokiej Izby na lawinowo rosnącą liczbę nielegalnych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom przewlekle chorym, niepełnosprawnym i w podeszłym wieku. 19 lipca tego roku Sejm dokonał nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Jednak wydaje się, że ten projekt, który wszedł w życie już w sierpniu, mimo wzrostu kar finansowych, mimo umożliwienia nakładania tzw. rygoru natychmiastowej wykonalności nie spowodował zmniejszenia liczby nielegalnie funkcjonujących placówek. W tych placówkach może dochodzić do wielu nadużyć. Takie przypadki były chociażby w Zgierzu, w Wolicy, w Trzciance. To są sytuacje kompletnie niedopuszczalne, w których mogą być nierespektowane prawa człowieka.

Panie ministrze, jakie działania podejmuje rząd, żeby usprawnić nadzór wojewodów nad tymi placówkami? Jak wygląda współpraca wojewodów z Policją, z samorządem gminnym?

Z upoważnienia prezesa Rady Ministrów odpowiedzi udzieli pan minister Marcin Zieleniecki. Proszę, panie ministrze. Wysoka Izbo!

Od razu mówię, że dane te nie potwierdzają na pewno tezy o lawinowym wzroście liczby placówek, które w sposób nielegalny zapewniają całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz osobom w podeszłym wieku. Myślę, że nawet teza o wzroście liczby takich placówek stoi też, że tak powiem, pod znakiem zapytania. Pragnę uspokoić pana posła: na pewno ze zjawiskiem lawinowego wzrostu liczby takich placówek nie mamy do czynienia. Ale odwołajmy się do danych statystycznych. Dane za ostatnie 4 lata.

Rok 2016 - cztery decyzje, rok 2017 - zero takich decyzji, rok 2018 - również zero, w 2019 r. wydano jedną decyzję nakazującą natychmiastowe wstrzymanie prowadzenia działalności. Mamy również dane dotyczące potencjalnej liczby nielegalnych placówek zapewniających całodobową opiekę w tym okresie.

Ta liczba utrzymuje się więc na mniej więcej stałym poziomie, tzn. ok. 100 takich placówek.

Podobny problem mają także województwa dolnośląskie, pomorskie i śląskie. Jeżeli chodzi o działania, jakie podejmują wojewodowie w sprawie placówek, które działają nielegalnie, to wojewoda, stwierdzając prowadzenie bez zezwolenia takiej placówki, może nałożyć karę pieniężną w wysokości 20 tys. zł, a w razie kontynuowania takiej działalności może zostać nałożona kara w wysokości 40 tys. zł. Pan poseł wspominał o tym, że 19 lipca 2019 r. Sejm uchwalił ustawę nowelizującą ustawę o pomocy społecznej. Część przepisów tej ustawy weszła w życie 4 października, część jeszcze nie zdążyła wejść w życie, dlatego że data wejścia w życie części przepisów to jest 1 stycznia 2020 r. Nowe przepisy przewidują m.in. możliwość nałożenia kary w wysokości 40 tys. zł na podmiot, który po otrzymaniu prawomocnie kary za prowadzenie bez zezwolenia jednej placówki przenosi ją w inne miejsce lub rozpoczyna prowadzenie innej placówki. Po to, aby przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi województwami przebiegał jak najsprawniej, wprowadziliśmy przepisy, które przewidują stworzenie specjalnego wykazu kar, który jest zasilany informacjami pochodzącymi od poszczególnych wojewodów. Ten wykaz jest następnie udostępniany wojewodom, którzy prowadzą postępowania w sprawie nałożenia kary albo wydania decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie (Dzwonek) takiej placówki. Dziękuję. Pytanie dodatkowe zada pani posłanka Monika Rosa. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Doskonale wiemy, że liczba wszczętych postępowań może nie oddawać pełnej skali funkcjonowania takich nielegalnych domów opieki nad seniorami. Stąd moje pytania. Czy państwo mają pomysł albo może wojewodowie, którzy mają obowiązek nadzoru nad domami zarówno działającymi legalnie, jak i tymi nielegalnymi, w jaki sposób kontrolować liczbę takich domów? W jaki sposób usprawnić przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi województwami, żeby rzeczywiście nie dochodziło do sytuacji przenoszenia z miejsca na miejsce takich nielegalnych placówek?

Dziękuję serdecznie pani posłance. Bardzo proszę, panie ministrze. Wysoka Izbo! Jeżeli chodzi o kwestie współpracy wojewodów z samorządami i z Policją w tym zakresie, to chcę powiedzieć, że oczywiście samorząd terytorialny to jest część systemu administracji publicznej, która jest odpowiedzialna za realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Tak że jest to ten szczebel struktury administracji publicznej, który na bieżąco monitoruje sytuację i ma, można powiedzieć, w zakresie obejmującym przedmiot naszej dyskusji najlepszy dostęp do informacji na temat tego typu placówek świadczących bezpodstawnie, bez podstawy prawnej tego typu działalność. Szczerze mówiąc, z informacji, jakich zasięgnęliśmy od urzędów wojewódzkich, nie wynikało, że są jakieś sygnały o braku dobrej współpracy czy, można powiedzieć, jakichś zakłóceniach, jeżeli chodzi o pozyskiwanie takich informacji i współpracę z samorządem terytorialnym w tym zakresie. Jeżeli chodzi o współpracę z Policją, to chcę zwrócić uwagę szanownych państwa posłów, że ta nowelizacja, o której wspominaliśmy, nie obejmuje wszystkich działań zmierzających do tego, aby ten system nadzoru i kontroli był jak najbardziej sprawny. Zwracam uwagę na przepisy karne, które pojawiły się w ustawie o pomocy społecznej.

Zwracam uwagę na przepisy Kodeksu karnego, które penalizują udaremnianie lub utrudnianie wykonania czynności służbowych osobie upoważnionej do przeprowadzania czynności w zakresie nadzoru i kontroli w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz osobom w podeszłym wieku. Chcę powiedzieć tak: 4 października to jest pierwszy termin wejścia w życie części tych nowych przepisów ustawy o pomocy społecznej, o których wspominałem, 1 stycznia to jest drugi termin. Zakładam, że te skutki będą pozytywne i liczba placówek nielegalnie prowadzących taką działalność spadnie. Jeżeli chodzi o informacje dotyczące województwa śląskiego. Już króciutko.

Dziękuję, panie ministrze. W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość pytanie w sprawie realizacji polityki senioralnej oraz dalszych planów i kierunków działań dotyczących podniesienia jakości życia polskich seniorów będą zadawały panie posłanki Joanna Borowiak, Barbara Bartuś, Lidia Burzyńska i Urszula Rusecka. Odpowiadał będzie sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pan minister Stanisław Szwed. Zgodnie z ustaleniami jako pierwszą poproszę panią Joannę Borowiak. Panie Ministrze! Seniorzy stanowią ważną grupę społeczną w Polsce, a ich doświadczenia zawodowe i życiowe są nieocenione dla każdego, szczególnie dla młodszych pokoleń. Jednym z priorytetów rządu Prawa i Sprawiedliwości jest spójna i kompleksowa polityka senioralna. To także ważny element realizacji strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Programy senioralne realizowane przez rząd są odpowiedzią na wyzwania, jakie stawia przed Polską polityka demograficzna i zachodzące procesy demograficzne. Zadaniem tych programów jest nie tylko poprawa warunków życia osób w srebrnym wieku, lecz także wykorzystanie ich potencjału i życiowego doświadczenia z korzyścią dla wszystkich. Ich najważniejsze cele to podniesienie jakości życia seniorów, umożliwienie im jak najdłuższej samodzielności, zapewnienie bezpieczeństwa i tworzenie warunków do podejmowania aktywności. Rząd w poprzedniej kadencji podjął szereg działań w tym zakresie. Należy tutaj wymienić takie programy jak: „Senior+”, „Leki 75+”, „Opieka 75+”, „Emerytura+”, „Mama 4+” czy wreszcie „Dostępność+” W trosce o nieustanną poprawę jakości życia osób starszych kierujemy do pana ministra pytanie:

Bardzo proszę. Dziękuję. Panie Marszałku! Panie Ministrze!

Dziękuję. Zapraszam pana ministra Stanisława Szweda.

Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję za to pytanie. Tematyka, którą panie poruszyły, jest bardzo ważna dla rządu Prawa i Sprawiedliwości.

Warto je przypomnieć.

Jeżeli ktoś ma niższą emeryturę ze względu na to, że nie wypracował sobie stażu emerytalnego, to ma dofinansowanie.

Tak że to też jest bardzo ważne rozwiązanie, oczywiście ono będzie kontynuowane. Program „Opieka 75+” kierowany jest do samorządu na wzmocnienie usług opiekuńczych.

W kontekście tego pytania pani poseł Bartuś dotyczącego wsparcia współpracy z opieką zdrowotną, z Ministerstwem Zdrowia - oczywiście też w tym zakresie jak najbardziej tak, później też programy czy świadczenie uzupełniające w kwocie 500 zł.

Program „Senior+” - z 50 mln wzrost nakładów do 80 mln. Kwota przeznaczona dla samorządów na tworzenie dziennych domów seniora+, klubów seniora+.

To jest program skierowany do organizacji pozarządowych, które mogą z tych programów skorzystać. Te programy cieszą się dużym uznaniem. Bardzo proszę o zadanie pytania. Dziękuję bardzo. Panie Ministrze! Obecnie w Polsce żyje ok. 9 mln ludzi, którzy mają 60+.

Dobrze, że żyjemy dłużej, natomiast wyzwania są również przed ministerstwem. Co zatem? Jakie zamierzenia wspierające osoby w srebrnym wieku i poprawiające jakość ich życia ma w planach Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej? Zapraszam serdecznie, panie ministrze. Panie Marszałku! Będziemy kontynuować te programy, o których mówię, bo to jest bardzo ważne.

Druga rzecz: kwestia waloryzacji. Utrzymujemy waloryzację procentowo-kwotową, aby te najniższe świadczenia wzrastały, były wyższe niż do tej pory.

Kontynuujemy program „Senior+”

Mamy nadzieję, że dzisiaj Sejm rozstrzygnie już o powołaniu, zamianie na Fundusz Solidarnościowy, gdzie również ta działka dotycząca emerytów, rencistów będzie miała duże znaczenie.

W ramach tych działań, które podejmujemy, wsparcie dla seniorów dotyczące ich materialnego bezpieczeństwa, uczestnictwa w życiu społecznym, aktywnego uczestnictwa, ale również tej solidarności międzypokoleniowej będziemy utrzymywać, wspierając finansowo.

Dziękuję serdecznie. Panowie posłowie z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość Waldemar Andzel, Andrzej Gawron oraz Jerzy Polaczek postanowili zadać pytanie w sprawie przeciwdziałania wypadkom na przejazdach kolejowych. Na to pytanie będzie odpowiadał sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury pan minister Rafał Weber. Wysoka Izbo! Pierwsza z nich to kategoria A, czyli miejsca z rogatkami lub bez nich. Przejazdy kategorii B dysponują półrogatkami oraz działającą samodzielnie sygnalizacją świetlną. Najgorzej zabezpieczone są przejazdy zakwalifikowane do kategorii D, bez rogatek i sygnalizacji świetlnej. Statystyki pokazują, że 99% wszystkich zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych wynika z niewłaściwych decyzji kierowców. Podstawowe błędy prowadzące do tragedii to ignorowanie znaku „stop”, przejeżdżanie pod zamykającymi się rogatkami, omijanie półrogatek. W związku z pojawiającymi się informacjami o tragediach, a szczególnie na niestrzeżonych przejazdach kolejowych, których w kraju jest sporo, i rosnącą liczbą ofiar zwracam się do ministra z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie: Jakie są przewidziane działania mające na celu zabezpieczenie bądź likwidację przejazdów niestrzeżonych? Czy jest znana dokładna liczba takich przejazdów, które nie są w żaden sposób zabezpieczone? Jakie są przewidziane działania w stosunku do kierowców, którzy lekceważą znaki i zamykające się rogatki? Proszę o odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury pana Rafała Webera. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję panom posłom za to pytanie. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ale też bezpieczeństwo przewozów kolejowych to nadrzędne cele działalności Ministerstwa Infrastruktury i możemy, bazując na tym pytaniu, powiedzieć o naszych działaniach, które podejmujemy w tym zakresie. Szanowni Państwo! Do głównych działań mających wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, które są realizowane przez Ministerstwo Infrastruktury, należy, po pierwsze, monitoring przejazdów. Na koniec 2018 r. mieliśmy 1343 przejazdy kolejowo-drogowe, które były wyposażone w monitoring. Po drugie, budowa skrzyżowań wielopoziomowych, czyli wiaduktów. Są one budowane przede wszystkich na tych liniach, na których docelowa prędkość pociągu wynosi albo będzie wynosić co najmniej 200 km/h.

W poprzedniej kadencji rządu Prawa i Sprawiedliwości wybudowaliśmy łącznie 395 skrzyżowań dwupoziomowych, a do końca obecnej kadencji, czyli do końca 2023 r., planujemy budowę kolejnych 417 wiaduktów. Chcemy w ten sposób unikać takiej bezpośredniej kolizji między jadącymi pociągami a samochodami. Po trzecie, modernizujemy istniejące przejazdy kolejowo-drogowe w kategorii D. Polega to na zmianie kategorii przejazdu na wyższą kategorię, a tym samym wyposażenie przejazdów w nowoczesne urządzenia zabezpieczające. Działania te wchodzą w zakres inwestycji kolejowych ujętych w krajowym planie kolejowym. W poprzedniej kadencji naszego rządu zmodernizowaliśmy łącznie 1737 przejazdów kolejowo-drogowych, a do końca obecnej kadencji planujemy modernizację kolejnych 1257 przejazdów kolejowych.

Przejazdy niepubliczne zabezpieczane są drągami odblaskowymi zamkniętymi na kłódkę, do której klucze posiada wyłącznie użytkownik, który zawarł z zarządcą infrastruktury kolejowej stosowną umowę.

Szanowni Państwo! Liczba przejazdów kategorii D zmniejsza się z roku na rok. Na koniec 2017 r. takich przejazdów było 6017, a na koniec 2016 r. było ich 7047, czyli w ciągu 2 lat zmniejszyliśmy, poprzez różnego rodzaju inwestycje, liczbę przejazdów kategorii D o blisko 500. Tak że bezapelacyjnie zwiększyliśmy bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o przejazdy kolejowo-drogowe. Jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie trzecie, jakie są przewidziane działania w stosunku do kierowców, aby nie lekceważyli prawa, to od 2005 r. PKP PLK prowadzą kampanię społeczną „Bezpieczny przejazd” Podstawowym zadaniem kampanii jest edukowanie uczestników ruchu drogowego poprzez podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych oraz kształtowanie zachowań i utrwalanie pożądanych postaw społecznych. W ramach kampanii PKP PLK organizują również seminaria dla instruktorów nauki jazdy. Tutaj znaczącą rolę odgrywa również UTK, czyli Urząd Transportu Kolejowego, który prowadzi kampanię społeczną „Kolejowe ABC” skierowaną do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich wychowawców i nauczycieli. Jednocześnie trwają prace przygotowawcze do pilotażowej instalacji urządzeń rejestrujących wykroczenia drogowe na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii B i C wskazanych przez PKP PLK w ramach systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym wykonywanego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. Ponadto chcę poinformować, że w październiku br. odbyło się spotkanie zorganizowane przez Urząd Transportu Kolejowego. Dotyczyło ono inteligentnego monitoringu przejazdów kategorii D z funkcją rejestracji wykroczeń polegających na ignorowaniu znaku B-20, czyli znaku „stop” Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pytanie dodatkowe zadaje pan poseł Andrzej Gawron, klub Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wspomniał pan, że jednym ze sposobów przeciwdziałania wypadkom na przejazdach kolejowych jest fizyczna likwidacja przejazdów, szczególnie tych mało uczęszczanych. Dotyczy to przejazdów kategorii D. Jednak wiąże się to również, panie ministrze, z utrudnieniami dla mieszkańców okolic, tych, którzy tam właśnie zamieszkują. Ja mam taki konkretny przykład z gminy Lubliniec, gdzie praktycznie kilka rodzin, jeżeli nastąpi likwidacja przejazdu kategorii D, zostanie odciętych od świata. Argumentacja jest taka, że droga, która przebiega przez tory, nie jest w ciągu drogi publicznej.

Wysoka Izbo! Staramy się indywidualnie, oczywiście w ramach prawa i w granicach prawa, podchodzić do każdego przypadku likwidacji przejazdu kolejowego kategorii D. Bardzo proszę pana posła, aby tym przypadkiem zainteresował mnie osobiście. Przeanalizujemy, jak tę sytuację możemy rozwiązać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Posłowie Jarosław Gonciarz i Wojciech Szarama, klub Prawo i Sprawiedliwość - pytanie w sprawie aktualizacji bazy pytań wykorzystywanych podczas egzaminu na prawo jazdy. Bardzo proszę, pan poseł Jarosław Gonciarz. Panie Ministrze! Wprowadzenie obowiązku utworzenia tzw. korytarzy życia ma zapewnić krótszy czas przejazdu służb ratowniczych do poszkodowanych, dla których nierzadko każda minuta, nawet sekunda jest bardzo ważna.

Pragnę jednak zwrócić uwagę na konieczność dokonania jej analizy w kontekście możliwości dostosowania obecnego zakresu nauki w szkołach jazdy do tych konkretnie, jak i innych przepisów. Podobnie jest z pytaniami na egzaminie teoretycznym, które powinny zostać zaktualizowane poprzez uwzględnienie wprowadzonych zmian.

Odpowiada sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury pan minister Rafał Weber. Wysoka Izbo! Jazda na suwak i korytarz życia to nowe obowiązki kierowców, które też przy udziale Wysokiej Izby zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego. Bardzo cieszymy się, że zostały one przyjęte przez kierowców w sposób pozytywny. Bez wątpienia zwiększają one bezpieczeństwo na polskich drogach. Bez wątpienia tworzenie korytarza życia przyspiesza przyjazd służb ratunkowych do miejsca wypadku i skraca czas udzielanej pomocy, natomiast jazda na suwak upłynnia ruch i powoduje, że zatory, które mogą się pojawiać przy zwężeniu jednego pasa ruchu i znikaniu jednego pasa ruchu, po prostu się nie tworzą. Cieszę się bardzo, że o tym cały czas trwa dyskusja, bo to zwiększa świadomość polskich kierowców, jeżeli chodzi o stosowanie się do tych przepisów Prawa o ruchu drogowym. Pan minister Andrzej Adamczyk od samego początku mówił, że będzie dążył do tego, aby pytania dotyczące suwaka i korytarza życia również były zawarte w zagadnieniach, w pytaniach egzaminacyjnych.

Oznacza to, że nawet najlepiej przygotowane osoby nie miały możliwości zapoznania się z zasadami ruchu drogowego określonymi w nowych przepisach. Dlatego też, mając to na względzie, chcemy zapewnić obecnym oraz przyszłym kandydatom na kierowców czas na to, aby się zapoznali z tymi przepisami, i podjęliśmy decyzję o tym, aby pytania egzaminacyjne w zakresie suwaka i korytarza życia wprowadzić za 3 miesiące. A więc po 3 miesiącach funkcjonowania tych przepisów prawa pojawią się w pytaniach egzaminacyjnych dla kierowców czy kandydatów na kierowców pytania związane z tworzeniem korytarza życia i jazdą na suwak. Bezapelacyjnie będziemy chcieli, aby kierowcy się do tych przepisów stosowali i tym samym zwiększali bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan poseł Wojciech Szarama ma dodatkowe pytanie? Bardzo proszę. Poprzednie pytanie było trochę prowokujące.

Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.

Składam wniosek w imieniu klubu koalicyjnego Lewica o ogłoszenie przerwy i zwołanie Konwentu Seniorów w celu przedyskutowania zmian w harmonogramie dzisiejszego posiedzenia.

Szanowni Państwo! To, co się wydarzyło wczoraj podczas obrad Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, woła o pomstę do nieba.

To jest ustawa fundamentalna, ustawa ustrojowa. To projekt, który wkracza w podstawowe funkcje działania państwa, i my mamy.

Ta ustawa w sposób fundamentalny zmieni filozofię działania polskich sądów. Podporządkuje te sądy władzy wykonawczej, zaknebluje usta polskim sędziom, połamie im kręgosłupy. Nie możemy w takim trybie, w trybie kilkunastu godzin, debatować i procedować nad tym projektem ustawy. Dziękuję.

Bardzo proszę, z wnioskiem formalnym pani Anna Żukowska, klub Lewicy. Składam wniosek formalny o skierowanie rozpatrywanego projektu ustawy o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw z powrotem do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka z tego powodu, że komisja nie miała wystarczająco dużo czasu na zapoznanie się z poprawkami zgłoszonymi przez wnioskodawców. Kilka poprawek nosiło ten sam numer. I tak naprawdę nie było wiadomo, kto je zgłasza, czy rzeczywiście posłowie wnioskodawcy, czy też te poprawki spływają z Ministerstwa Sprawiedliwości, którego przedstawiciele byli obecni podczas posiedzenia komisji. Również kluby parlamentarne, członkowie klubów, którzy nie są członkami Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, nie mieli okazji i nie mieli czasu zapoznać się z tym projektem oraz z poprawkami, ponieważ został on przyjęty w trybie zupełnie ekstraordynaryjnym pt. 10 godzin obrad Komisji Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Pan poseł Borys Budka z wnioskiem formalnym. Ja? Nie, pan poseł Borys Budka. Gdzie? Bardzo dziękuję. Panie Marszałku! W trybie art. 184 regulaminu Sejmu chciałbym złożyć wniosek formalny o przerwę, podczas której pani marszałek Sejmu, być może pan premier, udzieli szerszej informacji w zakresie listu Komisji Europejskiej, który został wystosowany i do pana premiera, i do pani marszałek, ale również, jak wskazują doniesienia, do prezydenta Andrzeja Dudy, i dotyczył zaniepokojenia Komisji Europejskiej tym wszystkich, co w ostatnich dwóch dniach dzieje się, jeśli chodzi o tzw. ustawę represyjną w zakresie polskich sędziów. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę, wniosek formalny, pan poseł Tomasz Trela, klub Lewica. Zrobimy to w bloku głosowań. Bardzo proszę. Panie pośle, pan raczy wykrzykiwać na sali. Wczoraj tutaj słyszeliśmy, że ci, którzy przygotowali ten projekt ustawy, sprawdzali, jak te przepisy funkcjonują w krajach Unii Europejskiej. Komisja Europejska wystosowała listy do pana premiera, do pana prezydenta, do pani marszałek Sejmu, do pana marszałka Senatu, żeby natychmiast wstrzymać pracę nad tą haniebną ustawą. Zgłaszam w imieniu klubu Lewicy wniosek formalny o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów celem omówienia jeszcze raz trybu procedowania nad tym projektem i przesunięcia go na kolejne posiedzenie Sejmu. Nie kompromitujcie Wysokiej Izby i nie kompromitujcie państwa polskiego, bo zaczynacie robić to po raz kolejny.

Natomiast jeżeli prawdą jest to, że Komisja Europejska skierowała do najważniejszych organów w Polsce bardzo mocny list z apelem o wstrzymanie prac nad tą kontrowersyjną ustawą, to jesteśmy w zupełnie innym miejscu, niż byliśmy nawet jeszcze dzisiaj nad ranem. Autorzy tego projektu zapewniali, jakoby rozwiązania w nim zawarte były zgodne z unijnym prawem, z prawem, które obowiązuje w innych krajach. Nic bardziej błędnego. Dlatego w imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej proszę pana marszałka o doręczenie posłom kopii listu Komisji Europejskiej skierowanego do marszałka Sejmu. W tym celu bardzo proszę pana marszałka o zarządzenie przerwy, by był czas dla klubów.

Panie i Panowie Posłowie! Wiem, że projekt ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych wywołuje wiele dyskusji, są listy. Ja nie o list poproszę, poproszę o elementarną przyzwoitość w procedowaniu, o doręczenie posłom opinii ministra spraw zagranicznych o zgodności tego projektu z prawem Unii Europejskiej.

Wszystkie autorytety stwierdzają, że zostało złamane prawo Unii Europejskiej. Niech wreszcie wypowie się minister spraw zagranicznych, to jest jego obowiązek. My wszyscy, panie i panowie posłowie, w tej Izbie tego się domagamy. Bardzo dziękuję.

Pani poseł Wanda Nowicka z wnioskiem formalnym. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Pani poseł, rozmawiamy o czymś, co nie jest w porządku obrad. Kiedy nie ma pieniędzy na organizacje działające na rzecz praw kobiet, zawsze znajdą się pieniądze na telewizję propagandową.

Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 69 i 107)

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka nałożyła na mnie obowiązek, ale i zarazem przywilej przedstawienia raportu z prac komisji dotyczących procedowanego aktu normatywnego. Pozwolę sobie zatem w sposób esencjonalny i skondensowany przedstawić w tym zakresie stosowne informacje. W toku prac zgłoszono ponad 100 poprawek. Komisja pozytywnie zaopiniowała 22 poprawki, które uszlachetniają pierwotny projekt ustawy.

Komisja rekomenduje przyjęcie ustawy w kształcie uwzględniającym pozytywnie rozpatrzone poprawki. I kwestia techniczna.

W sprawozdaniu komisji zaszła oczywista omyłka pisarska. Wyraz „dyscyplinarnie” należy zastąpić wyrazem „dyscyplinarne”

Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.

Mój klub przystaje na to. Jako pierwszy w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość pan poseł Przemysław Czarnek. Bardzo proszę. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Przecież z jednej strony mówiliście państwo, że nie możecie pracować w takim tempie, że nie mieliście szansy zapoznać się z projektem ustawy, a zwłaszcza z poprawkami, które były składane. Nagle słyszymy, że Komisja Europejska wystosowała pismo do najwyższych organów władzy Rzeczypospolitej Polskiej, w którym wyraża zaniepokojenie projektem i poprawkami. Komisja miała szansę, żeby zapoznać się tak głęboko z projektem i poprawkami, a państwo nie mieliście? Nie płacą wam za siedzenie, tylko za czytanie i analizowanie tego, co jest przedmiotem pracy Wysokiej Izby. Panie Marszałku! Historia doktryn politycznych i prawnych zna różne mutacje czegoś, co nazywamy państwem prawa, państwem praworządnym. Każda z tych mutacji jest niedobra, każda z tych mutacji osłabia praworządność. Najbardziej jednak osłabia praworządność mutacja, którą nazywamy państwem sędziów. Państwo sędziów to jest dokładnie to państwo i ten model, do którego państwo dążycie i który państwo chcecie wprowadzać od 3 tygodni przy pomocy posłusznych sobie sędziów. Państwo sędziów to państwo, które ignoruje zasadę suwerenności narodu, ignoruje zwierzchnictwo narodu nad wszystkimi trzema władzami. Państwo sędziów to państwo, w którym sędziowie decydują o tym, co jest prawem, a co nie jest. Wczoraj w nocy też to słyszeliśmy. Sędziowie uzurpują sobie prawo do tego, żeby stwierdzać, kto jest sędzią, a kto nie. Wczoraj w nocy też o tym słyszeliśmy. Pytanie, skąd ta aberracja i skąd ta przewrotność. Szanowni Państwo! To nie my zainicjowaliśmy ten szybki proces legislacyjny. To państwo go zainicjowaliście. To państwo podcięliście żyły polskiemu porządkowi prawnemu i ładowi konstytucyjnemu. Musimy ten plaster na tę ranę przykleić, bo nie możemy pozwolić na to, żeby wykrwawił się polski porządek prawny. Czego wy chcecie? Wy chcecie podłożyć bombę pod polski ład konstytucyjny, powołując się na konstytucję. Rzeczywiście wczoraj w nocy i dzisiaj nad ranem odbywały się obrady Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. One były niezwykle pouczające. Bardzo trudne, bardzo męczące, ale przecież jesteśmy dla społeczeństwa i nikt z nas nie narzeka, oprócz niektórych posłów opozycji. Ale to były bardzo pouczające obrady. Myśmy dostrzegli podczas tych obrad jedną bardzo ważną rzecz. Otóż problem jest większy, niż myśleliśmy.

Ludzie żądają wręcz od nas, żebyśmy zastopowali łamanie konstytucyjnego ładu i konstytucyjnego porządku prawnego w Polsce.

To wy chcecie wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. To wy kablujecie do Komisji Europejskiej. To wy kłamiecie na temat Polski. To wy kłamiecie ma temat społeczeństwa polskiego. My wam na to nie pozwolimy. Nie damy się wypchnąć z Unii Europejskiej. Szanowni Państwo! Straszycie kilka dni przed Bożym Narodzeniem Polaków jakimś urojonym systemem, w którym będzie się podważać kilkadziesiąt tysięcy, a może kilkaset tysięcy wyroków prawomocnie wydanych przez legalnie orzekających sędziów w tym kraju. To jest straszenie Polaków. To jest tak naprawdę zamach na praworządność. Dlatego właśnie, szanowni państwo, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, panie i panowie posłowie Prawa i Sprawiedliwości doprowadzą do tego, że dzisiaj ta ustawa będzie uchwalona, bo ten plaster na ranę, którą zrobiliście, musi być przyczepiony. Ratujemy praworządność w Polsce. Bardzo dziękuję. Pan poseł Jacek Ozdoba, klub Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Cały czas to chyba, jak widać, robicie. Co prawda mam tutaj trochę takie déja vu, jak patrzę na was, bo kilka lat temu również opowiadaliście Polakom, jak to jest strasznie i w ogóle, próbowaliście to wszystko zablokować, po czym okazało się, że to był pic na wodę, fotomontaż, brakuje tylko

Widzą scenariusz: przemawia polityk, a później przemawia sędzia, który za chwilę będzie orzekał w jego sprawie. Ten sędzia wyklucza się z zawodu.

kpinę z poważnego projektu, który jest oczekiwany przez Polaków, kpinę z projektu, który. Ja pani coś powiem, coś pani zacytuję, pani koleżankę: Nie, Kamila, nie jesteś tu sama, nie. Ja rozumiem, że jest pani reprezentantem osób, które... ma pani być tutaj osobą, twarzą jakby przeciwstawiania się tej „strasznej”, dobrej ustawie.

Wysoka Izbo!

na rzecz państwa polskiego wymaga, żeby sobie z poważnych rzeczy jaj nie robić, żeby przyjmować ustawy nawet wtedy, kiedy są trudne, ale są wymagane. bo muszą przeciwdziałać anarchizacji polskiego życia publicznego. I poważna praca na rzecz państwa polskiego wymaga tego, aby składać poprawki, które poprawiają te ustawy realnie, które eliminują zagrożenie stwierdzenia niezgodności z prawem europejskim, które usuwają niepotrzebne regulacje. Rzeczywiście w pierwotnym projekcie były regulacje, które odnosiły się do tego, że sędziowie byliby zobowiązani składać chociażby oświadczenia w zakresie swoich aktywności w Internecie. Usunęliśmy te zapisy. Usunęliśmy zapisy, które mogą być sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. dodaliśmy preambułę, która w sposób jasny określa podstawy aksjologiczne stojące u podstaw konieczności przyjęcia tego projektu. Nie możemy pozwolić sobie na destabilizację państwa. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka obradowała wczoraj i dzisiaj, w dużej mierze dzięki państwu, dzięki państwa wnioskom, które się pokrywały, były takie same. Wykorzystywaliście państwo czas do maksimum, argumentowaliście w sposób absolutnie powtarzalny tylko po to, by przeciągnąć prace komisji w czasie, aby Polakom wmawiać, że posłowie Zjednoczonej Prawicy pracują nocami. Jak trzeba, pracujemy nocami. Ja się bardzo cieszę, że Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka przyjęła wszystkie wnioski Porozumienia Jarosława Gowina, i w imieniu parlamentarzystów Porozumienia Jarosława Gowina deklaruję wsparcie dla tej ustawy. Bardzo dziękuję. Teraz głos ma pan poseł Borys Budka.

W imieniu klubu parlamentarnego, panie marszałku, składam w ramach drugiego czytania trzy poprawki do tego projektu ustawy, poprawki o charakterze głównie technicznym. Istotą pierwszej poprawki jest użycie wyrazów: działanie i zaniechanie w liczbie pojedynczej zamiast liczby mnogiej, druga poprawka ma na celu przekazanie do wyłącznej właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego spraw skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Sądu Najwyższego, jeżeli chodzi o podważenie legalności działania sędziego, a trzecia poprawka ma na celu objęcie dyspozycją przepisu również wniosków o oznaczenie sądu, przed którym ma się toczyć postępowanie, składanych na podstawie art. 45 Kodeksu postępowania cywilnego.

Teraz głos ma pan poseł Borys Budka w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Będę powtarzał do skutku: nie było i nie ma żadnej reformy wymiaru sprawiedliwości.

Dokładnie w ten sam sposób potraktowaliście polską służbę zdrowia, system edukacji, szkolnictwo wyższe, jak i sądownictwo. Udajecie wielkich reformatorów, a wszędzie wprowadzacie jeden wielki chaos. Nie potraficie sprawić, by postępowania sądowe były szybsze, zablokowaliście de facto drobne postępowania prokuratorskie, bo prokuratorzy boją się wydawać jakiekolwiek postanowienia tylko dlatego, że mają ten politnadzór ze strony ministra sprawiedliwości, a teraz ten chaos, który wprowadziliście w Krajowej Radzie Sądownictwa, w Trybunale Konstytucyjnym i w sądach powszechnych, próbujecie zamienić w większy jeszcze chaos. Okłamujecie Polki i Polaków, twierdząc, że jesteście Europejczykami i rozumiecie, na czym polega Wspólnota Europejska, podczas gdy tak naprawdę wprowadzacie do polskiego porządku prawnego rozwiązania typowe dla krajów totalitarnych, gdzie to politycy mogą. Jak działacie w praktyce? Otóż w praktyce minister sprawiedliwości potrafi odwołać z delegacji sędziego tylko dlatego, że nie zgodził się na tymczasowe aresztowanie, o które wnioskował prokurator podległy temu samemu ministrowi. Nie chodzi wam o Polskę, nie chodzi wam o Polaków, nie chodzi wam o to, żeby cokolwiek zmieniać na lepsze - wam chodzi o bezkarność. Wy po prostu marzycie, by z kolejnej instytucji stworzyć to, co Marian Banaś stworzył zarówno w swojej kamienicy, jak i w Najwyższej Izbie Kontroli. Symbolem tego, w co zamieniliście państwo polskie i wymiar sprawiedliwości, jest ta kamienica Banasia. I tylko dlatego że jesteśmy w parlamencie, będę używał synonimu, a nie będę mówił tego słowa, co zrobiliście z wymiarem sprawiedliwości. Bezkarność, bezkarność, bezkarność - to jest jedyny cel, który przyświeca waszemu projektowi ustawy. Okłamujecie Polki i Polaków, twierdząc, że są to europejskie rozwiązania. Siedem zarzutów... ...podczas gdy Komisja Europejska w bardzo twardym stanowisku mówi wyraźnie: proszę zaprzestać prac nad tym haniebnym projektem, bo Polska, Polacy stracą pieniądze europejskie. Ale tak naprawdę wam chodzi o polexit. Wiecie dlaczego? wy nie znosicie jakiejkolwiek kontroli. Wy genetycznie boicie się jakichkolwiek niezależnych instytucji. Dlatego tak nienawidzicie Komisji Europejskiej, bowiem ta Komisja przejęła rolę i działa w interesie Polek i Polaków, podczas gdy ten rząd chce Polki i Polaków podporządkować kagańcowi władzy. Obiecaliście wielką reformę, a tak naprawdę zepsuliście wszystko, nawet to, co działało dobrze. Doprowadziliście wymiar sprawiedliwości do ruiny tylko po to, by teraz udawać, że go naprawiacie, a wprowadzacie kaganiec. Przecież to, co zrobiliście z Trybunałem Konstytucyjnym, jest najlepszym przykładem, jak działają wasze pseudoreformy. Zablokowaliście totalnie działanie tego organu, a pseudoprezesem zrobiliście odkrycie towarzyskie, jak mówi wasz prezes - częściej gotuje obiady, niż zajmuje się orzekaniem, jak to ktoś wczoraj powiedział. To jest prawdziwy obraz wymiaru sprawiedliwości. I teraz chcę, szanowni państwo, zapewnić o jednym. Nie poprzestaniemy na tym, co w tej chwili stało się w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Nawet zabieraliście najbiedniejszym z PCK, wasz były poseł jest oskarżony. Polacy nie zapomną wam tego, że niszczycie dorobek polskiej wolności.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Posłanki i Posłowie PiS-u! Budujecie piramidę bezprawia, a ta ustawa represyjna jest jej kolejną warstwą. Po wprowadzeniu tej ustawy rząd będzie mógł usunąć każdego sędziego pod byle pretekstem. Sędziowie będą karani za stosowanie polskiej konstytucji i unijnych traktatów. Powstrzymajcie prace zgodnie z apelem Komisji Europejskiej. Nie wyrzucajcie Polski z Unii Europejskiej. Wysoka Izbo! To politycy PiS wywołali pożar, który w tym momencie trawi system prawny w Polsce. I zamiast go ugasić zgodnie z zaleceniami unijnego Trybunału, podlewacie go tylko benzyną, proponując ustawę o dyscyplinowaniu sędziów. Ostrzegaliśmy wielokrotnie przed tym, że zmiany, które obecna władza wprowadza od 4 lat, ograniczając niezależność sądownictwa, wywołają chaos prawny. I to się dzieje na naszych oczach, z winy polityków PiS-u, a ustawa, którą dzisiaj proponujecie, tylko pogłębia ten chaos prawny. Posłanki i Posłowie PiS-u! Budujecie piramidę bezprawia. Ale ona przetrwa tylko do momentu, do którego będziecie rządzić, a potem się zawali. Tylko że pod gruzami tej piramidy bezprawia będą zwykli ludzie. Niestety PiS, niszcząc sądownictwo, niszczy życie zwykłym ludziom, niszczy możliwości działania polskim firmom. Wyroki sądów PiS, obsadzonych przez neo-KRS, będą warte tyle co makulatura. Z czasem będą po prostu kolejno podważane. Dlatego dla ludzi, dla przedsiębiorców taki wyrok będzie po prostu bezwartościowy. Taki wyrok będzie wyłącznie źródłem problemów w przyszłości. Moje pokolenie sytuację, w której prokurator ściga niezależnego sędziego za to, że on stosuje prawo, zna tylko z historii, może z opowiadań rodziców. Ja sama urodziłam się jeszcze w PRL, ale dzięki odwadze, bohaterstwu takich ludzi, jak Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki. Jacek Kuroń i wielu, wielu innych, miałam to ogromne szczęście, by w dorosłość wchodzić w wolnej Polsce. Dzięki ciężkiej pracy i zdecydowaniu takich ludzi, jak Leszek Balcerowicz i wielu, wielu innych. moje pokolenie dostało szansę życia w Polsce, która jest najbogatsza w swojej dotychczasowej historii. Dzięki takim ludziom, jak Jerzy Buzek, Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Geremek i wielu, wielu innych. Ale z powodu takich ludzi, jak Andrzej Duda, pan Zbigniew Ziobro, pan Jarosław Kaczyński, możemy to wszystko stracić w ciągu kilku najbliższych lat. Możemy stracić to wszystko, co w ciągu ponad ćwierć wieku polskiej wolności budowały kolejne pokolenia ludzi prezentujących pełną paletę poglądów i wrażliwości. Budowały nie dla siebie, budowały dla 38 mln Polaków i dla następnych pokoleń. Niszcząc niezależność polskich sądów, niszczycie warunki do dalszego bogacenia się Polek i Polaków. Niszcząc niezależność polskich sądów, niszczycie miejsce i przyszłość Polski w Unii Europejskiej.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! No cóż, minęło kilkanaście godzin od pierwszego czytania, a my dzisiaj rano już mamy sprawozdanie komisji.

Komisja, która wczoraj obradowała całą noc, aż do samego rana rozjeżdżała polskie sądy. Pod osłoną nocy, bez możliwości zabrania głosu przez organizacje pozarządowe i przedstawiciela rzecznika praw obywatelskich. Dzisiaj chciałbym powitać pana Adama Bodnara, rzecznika praw obywatelskich, na naszej sali. Nie pozwoliliście na wysłuchanie publiczne, a przecież to jest ustawa, nad którą właśnie powinno debatować szerokie grono reprezentantów społeczeństwa, organizacji pozarządowych w ramach wysłuchania publicznego. Pan poseł sprawozdawca powiedział, że zgłoszone wczoraj na posiedzeniu komisji poprawki uszlachetniły ten wspaniały projekt. No tak, uszlachetniły na takiej samej zasadzie, jak uszlachetnia cierpienie. Rzeczywiście trzeba przyznać rację. Ja się tak zastanawiam, czego się baliście, że przez te parę godzin aż do 5.30 rano pracowaliśmy w tej komisji. Że ludzie zobaczą wasze prymitywne fortele, które przemycacie tym projektem? Że społeczeństwo się dowie, że zakazujecie polskim sędziom orzekać na podstawie polskiej konstytucji? A może boicie się prawdy o tym, że planujecie zamach na Sąd Najwyższy i w efekcie wprowadzonych nowych procedur chcecie doprowadzić do tego, żeby pierwszym prezesem Sądu Najwyższego być może został partyjny nominat z Izby Dyscyplinarnej, który przecież nawet nie jest sędzią, jak orzekły ostatnio sądy? Ta ustawa to zwykły, prymitywny bubel prawny, który ma być narzędziem stosowanym przez podobnych wam partyjnych aparatczyków w państwach autorytarnych. Tam właśnie władza decyduje o tym, który wyrok jest zgodny z prawem i który jest sprawiedliwy. Gratuluję wzorców do naśladowania. Zapewniam wielu z was, że wielu opozycjonistów także z poprzedniego systemu, walczących o prawo obywateli do uczciwego procesu i sprawiedliwego wyroku, jest wstrząśniętych, widząc, że próbujecie to konstytucyjne prawo odebrać obywatelom. Jestem też przekonany, że przeciwko waszym działaniom pierwszy zaprotestowałby prof. Lech Kaczyński, który wielokrotnie podkreślał najwyższą wartość rządów prawa. PiS, wprowadzając taki przepis, nie martwi się o prawa zwykłych Polaków. Część z tych orzeczeń może być. Akurat prezydenta Lecha Kaczyńskiego niezmiernie szanuję i korzystałem wielokrotnie z jego dorobku naukowego, więc proszę się uspokoić, pani posłanko. Pozbawiacie obywateli ich podstawowego prawa człowieka, jakim jest prawo do niezależnego, bezstronnego sądu i uczciwego wyroku. Chcecie zamienić sędziów w maszynki do wydawania wyroków pod dyktando Nowogrodzkiej i na podstawie PiS-owskich przepisów. A może po prostu chcecie doprowadzić do tego, żeby sędziowie zamienili togi sędziowskie na partyjne uniformy? Może powiedzcie to wprost. Proponuję, żeby nie bawić się w tej Izbie w udawanie procesu legislacyjnego, a po prostu wyciąć kilka tysięcy tekturowych postaci Jarosława Kaczyńskiego, postawić je za sędziowskimi stołami, a w całej Polsce efekt będzie taki sam. Szkoda, że przed wyborami nie mieliście odwagi zaprezentować projektu tej ustawy. Szkoda, że nie mówiliście wtedy, że Piotrowicz i Pawłowicz będą w Trybunale Konstytucyjnym. Jesteście po prostu tchórzami, którzy wykonują bezwolnie każde polecenie waszego generała. Wy pod ten fundament państwa prawa podkładacie właśnie dynamit. Dlaczego to robicie? Ja wam powiem. Bo wy się po prostu boicie. Boicie się utraty władzy, boicie się, że wasze krętactwa ujrzą światło dzienne, boicie się trupów w szafie takich jak Banaś czy Chrzanowski. Boicie się, że sądy mogłyby orzekać i skazywać waszych kolesi, kolesi także z ław poselskich i rządowych. Jesteście po prostu tchórzami. A ta ustawa ma być polisą ubezpieczeniową waszej bezkarności. Jeżeli myślicie, że polscy sędziowie ze strachu przed wami porzucą rotę ślubowania i zamienią sędziowskie togi na drelichy partyjnych aparatczyków, to znaczy, że mierzycie ich własną miarą. To znaczy, że nie znacie hartu ducha polskich sędziów. Dziękuję.

Wysoka Izbo! Prawo i Sprawiedliwość dobrze wie, że wywołało pożar ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Izbie Dyscyplinarnej.

Proponuje, aby szanować tak naprawdę wybór sędziów przez tę neo-KRS, upolitycznioną KRS, KRS, która została powołana ze skróceniem kadencji poprzedniej Krajowej Rady Sądownictwa, i chce spowodować, żeby zrobić taki deal - bo to jest w tej ustawie - że za cenę szanowania, uznania, że sędziowie, którzy zostali wybrani przez Radę Państwa, są dalej sędziami, chce uznać, że także ci sędziowie, którzy są wybrani przez nową KRS, również są prawomocnie wybranymi sędziami. Takiego dealu nie będzie. Każdy sędzia w każdym przypadku powinien być oceniany indywidualnie i jego wybór także powinien móc być oceniany indywidualnie. Nie powinno być możliwości, że pierwszym prezesem Sądu Najwyższego zostanie osoba wyłoniona ze składu tej izby, bo de facto do tego sprowadza się kolejne, czyli najmniejsze, kworum przewidziane przez tę ustawę. Nie ma też zgody na to, żeby funkcjonowało w obiegu prawnym takie stanowisko jak pełniący obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Dlatego że taka osoba miałaby możliwość przewodniczenia Trybunałowi Stanu, brania udziału w posiedzeniach Sejmu, bycia członkiem KRS, a także mogłaby wybrać trzech członków Państwowej Komisji Wyborczej. Osoba, która - podkreślam - nie pełni funkcji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.

Szanowna Pani Marszałek! Panie Marszałku! W imieniu Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy na podstawie art. 45 zgłaszam wniosek o odrzucenie projektu ustawy o zmianie Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. W przypadku odrzucenia powyższego wniosku zgłaszam następujące poprawki w drugim czytaniu do sprawozdania komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, na posiedzeniu Sejmu RP.

1. Sędzia jest obowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o posiadanym wykształceniu. Art. 107 § 1: Za przewinienia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa i uchybienia godności urzędu, przewinienia dyscyplinarne, sędzia odpowiada dyscyplinarnie przed właściwym sądem.

Odwołania wniesione przez uczestników postępowania podlegają rozpoznaniu oddzielnie. Za przewinienia służbowe, w tym za oczywistą, rażącą obrazę przepisów prawa i uchybienia godności urzędu, prokurator odpowiada dyscyplinarnie przed właściwym sądem, o którym mowa w art. 145. Miło jest Wysokiej Izbie słuchać w takim trybie wnoszonych poprawek?

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Chciałbym w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15 przedstawić nasze refleksje na temat - nie boję się użyć tego sformułowania - tzw. ustawy represyjnej. Na początku powiem tak: szanowny panie ministrze, panowie i panie, panie i panowie posłanki z PiS-u, udało wam się. Udało wam się zrobić piorunujące wrażenie na wielu Polakach w Polsce, ale widzę, że to wrażenie jest równie piorunujące poza granicami Polski. Myślę, że powinniście się wszyscy, powinniśmy się wszyscy zacząć obawiać skutków tego wrażenia.

Nie tak dawno - warto przypomnieć - w swoim exposé pan premier Morawiecki wielokrotnie wspominał o nadchodzącej normalności, a takie stanowienie prawa niestety z tą normalnością ma niewiele wspólnego.

Ale wczoraj było widać jak w soczewce, że duch pana przewodniczącego prokuratora Piotrowicza cały czas unosi się nad Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Mówicie państwo o potrzebie reformy wymiaru sprawiedliwości.

Pytam się dzisiaj, po ponad 4 latach rzekomego realizowania oczekiwań Polek i Polaków, co mają Polacy po waszych reformach? Mają. Na pewno mają. Mają, mają.

Trochę statystyk, jeśli chodzi o wasze reformy, które tak często lubicie przywoływać. 2018 r. - chluba, wasz sztandarowy projekt - Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która miała być receptą na wszelką niesprawiedliwość w wymiarze sprawiedliwości.

Idźmy dalej. Kolejny sztandarowy pomysł w ramach reform wymiaru sprawiedliwości według PiS - Izba Dyscyplinarna. Była tak zachwalana przez PiS, a była jeszcze lepsza, bo w 2018 r. - uwaga - rozpatrzyła zaledwie 19% spośród spraw, które do niej wpłynęły.

Proszę spokojnie. Jarosław, nic nie mogę.